Wysoka Izbo! Na podstawie art. 184 ust. 2 i 3 regulaminu Sejmu składam wniosek o przerwę w posiedzeniu Sejmu w celu zwołania Konwentu Seniorów i dodania do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu ustawy, który złożyła Lewica i który od kilku dni nie jest procedowany, co wiąże się z zapewnieniem 75-procentowego dofinansowania miejsc pracy każdego Polaka i każdej Polki. Dzisiaj od rana Polacy są świadkami haniebnych targów, haniebnych deali pomiędzy panem premierem Gowinem a panem premierem Kaczyńskim. Ta Izba powinna zajmować się porządną pracą na rzecz Polaków, którzy dzisiaj masowo tracą pracę, natomiast dzisiaj Jarosław Gowin proponuje zmianę konstytucji, zmianę ustawy zasadniczej. Przypominam, że ta konstytucja jest nie tylko na dobre czasy, ale także na złe czasy, i nie czas na grzebanie przy konstytucji, nie czas na majstrowanie przy ustawie zasadniczej.

Dobrze, w takim razie, ponieważ został zgłoszony wniosek o przerwę, przystąpimy do głosowania. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.

Wznawiam obrady.

Kłaniam się, szczęść Boże. Wysoka Izbo! Wnoszę o odroczenie obrad Sejmu do czasu przywrócenia im należytej powagi przez panią marszałek. To jest kompletnie niepoważne - zwoływać Wysoką Izbę, wywieszając jednocześnie plan pracy na najbliższą godzinę i ogłaszając, że ta praca zostanie znowu przerwana po to, żeby pani marszałek dowiedziała się, jaki jest dalszy ciąg scenariusza, w którym pani marszałek skądinąd odgrywała jedną z pierwszoplanowych ról, ale nie jest wtajemniczona w pełną dramaturgię tych zdarzeń i dlatego musi się dowiadywać co jakiś czas, co ma być. A więc ogarnijcie się, szanowni państwo, nie rozbudowujcie tej sceny cyrkowej w gmachu Sejmu.

Nie, panie pośle, w takim razie nie poddam tego wniosku pod głosowanie, ponieważ jest on tożsamy z wnioskiem, nad którym głosowaliśmy przed chwileczką. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad do poniedziałku.

Jest to jedyna konstytucyjna możliwość na usankcjonowanie tego bezprawia, które w tej chwili ma miejsce. Bardzo proszę panią marszałek o wprowadzenie do porządku obrad ustawy, która gwarantuje odszkodowania wszystkim tym, którzy od dłuższego czasu są pozbawieni możliwości zarobkowania i którzy tracą pracę. Straciliśmy kilka godzin na wasze przepychanki.

Został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie posiedzenia do poniedziałku. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia do poniedziałku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Wniosek został odrzucony. Komisja Finansów Publicznych przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., druk nr 315.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (druki nr 313 i 315) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 regulaminu Sejmu, skierował w dniu 31 marca tego roku powyższy projekt do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania. W tym pierwszym czytaniu rządowego projektu, który zawiera 35 artykułów, zostały złożone cztery poprawki, które dotyczyły albo całkowitego, albo częściowego zmienienia tych zapisów.

Po merytorycznej dyskusji i głosowaniu Komisja Finansów Publicznych występuje i wnosi do Wysokiej Izby o uchwalenie załączonego projektu ustawy. Dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Panie Premierze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., druk nr 313, i sprawozdania Komisji Finansów Publicznych, druk nr 315. Jest to ustawa na obecny czas niezbędna ze względu na realizację programów z wykorzystaniem środków europejskich, realizację programów operacyjnych. W związku z trudnościami, jakie pojawiły się we wdrażaniu, w realizacji tych programów w związku z epidemią, konieczne jest, aby beneficjenci nie ponosili z tego tytułu konsekwencji dotyczących różnych spraw, m.in. terminów składania wniosków, rozliczeń, ale też sposobu prowadzenia projektów.

Jest to niezwykle potrzebny zapis ustawowy ze względu na to, że w momencie braku takiego zapisu i występowania tych okoliczności wielu beneficjentów mogłoby mieć z tego tytułu wiele problemów.

To upoważnienie, szczególnie np. w odniesieniu do samorządów, które są gospodarzami regionalnych programów operacyjnych, pozwoli na to, by te środki zostały przekazane, oczywiście również w drodze wyjątku.

To są te wszystkie zapisy, które są niezwykle istotne, przede wszystkim dla dobra beneficjentów. Ustawa przewiduje również zmianę harmonogramu realizacji projektów po to, żeby ten program można było zaktualizować w związku z czasem trwania epidemii.

Jest również specjalny tryb naboru wniosków dla instytucji zarządzających, w przypadku kiedy te wnioski będą dotyczyły przeciwdziałania skutkom epidemii.

Nie zmieniają one oczywiście ogólnych zasad i rygorów ustawy o wykorzystaniu środków unijnych. Dlatego też klub Prawo i Sprawiedliwość popiera ten projekt ustawy i wnosi o jego jak najszybsze uchwalenie. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Borysa Budkę, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo! Polscy pracownicy oczekują konkretnych rozwiązań, pracodawcy zamykają swoje zakłady tylko i wyłącznie dlatego, że zamiast z prawdziwą tarczą antykryzysową mamy do czynienia z wielką fikcją. Nie posłuchaliście państwo nas tutaj, w Sejmie, nie posłuchaliście dobrych rad Senatu i odrzuciliście wszystkie poprawki. Dzisiaj debatujemy nad ustawą, która w takiej maleńkiej części stara się załatać to, co zrobiliście, natomiast nie rozwiązuje istoty problemów. Dzisiaj polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy potrzebują tego, by traktować ich uczciwie i po partnersku. Dzisiaj państwo nie może bez zaufania do swoich obywateli nieść pomocy. Proponowaliśmy i proponujemy: zastąpmy wszystkie rygory formalne oświadczeniami, zaufajcie wreszcie polskim pracownikom i pracodawcom, zaufajcie obywatelom i pozwólcie im utrzymać ich miejsca pracy. Wreszcie upominamy się o polskich lekarzy, upominamy się o polskie pielęgniarki, upominamy się o służbę zdrowia. W Sejmie leży projekt ustawy, który gwarantuje wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, osobom, które walczą z koronawirusem, cotygodniowe testy. Kolejne szpitale są wyłączane tylko i wyłącznie dlatego, że nie potraficie państwo zrozumieć, że bezpieczeństwo zdrowotne to jest rzecz najważniejsza. Po raz kolejny apeluję do pana: niech pan wreszcie usiądzie do rozmów o tym, jak pomagać polskim pracownikom, jak pomagać polskim pracodawcom. Ludzie tracą pracę, zostają bez zasiłków, zostają bez pomocy, a wy ciągle bawicie się w wybory. Straciliśmy dzisiaj kilka godzin tylko dlatego, że próbujecie rozgrywać między sobą to, co się w tej chwili dzieje. Skupmy się na wspólnej pracy, zróbmy wspólnie coś dobrego dla Polski i Polaków, a później, gdy minie czas epidemii, przyjdzie czas na rozstrzygnięcia wyborcze. Im wcześniej to zrozumiecie, tak jak zrobił to pan premier Gowin, tym lepiej dla was, ale też lepiej dla Polski. Dziękuję, panie pośle, choć to nie jest punktem tego porządku. Panie Premierze!

Z tego Polska może mieć nawet 50 mld zł, czyli więcej, niż dotychczas wyskrobał ze wszystkich źródeł rząd - dużo więcej. Ale jest jeden warunek: te środki muszą być lepiej wykorzystane niż dotychczas. Przed chwilą słyszeliśmy, panie premierze, że polska służba zdrowia jest gotowa do walki z koronawirusem, a dzisiaj wiemy, że co szósty zakażony to pracownik opieki zdrowotnej. Dodatkowo 4,5 tys. członków personelu medycznego nie może nas leczyć, bo przebywa właśnie na kwarantannie. Za chwilę to samo zrobicie z polską gospodarką. W ostatnich trzech dniach marca zlikwidowano lub zawieszono w Polsce działalność 22 tys. firm. To jest odpowiedź przedsiębiorców na waszą dziurawą tarczę. Jeśli ktoś jeszcze w Polsce myśli, że polscy przedsiębiorcy - niezależnie od tego czy mali, czy średni, czy duzi - leżą na pieniądzach, to niech natychmiast przestanie w ten sposób myśleć. Nie leżą, panie premierze. Polscy przedsiębiorcy, którzy z dnia na dzień musieli zaprzestać swojej działalności na mocy waszej decyzji, dzisiaj patrzą bardzo często na swoje puste konta w bankach i zastanawiają się, z czego zapłacą pracownikom, kontrahentom i państwu, bo państwo nie chce ich nawet zwolnić ze składek na ZUS. Jak dziś ich z tych składek nie zwolnimy, to za dwa, trzy miesiące ZUS i tak ich nie dostanie, bo ci przedsiębiorcy po prostu upadną. Nad czym dzisiaj zastanawiają się przedsiębiorcy? Jeśli dziś stracą płynność, będziecie za to odpowiedzialni, bo oni za chwilę, kiedy sytuacja wróci do normalnego stanu, nie będą mieli za co wznowić swojej działalności gospodarczej. To są dylematy polskich przedsiębiorców. Te środki unijne trzeba dobrze wykorzystać. Jako przewodnicząca podkomisji ds. weryfikacji wykorzystania środków unijnych obiecuję wszystkim Polkom i Polakom, że rozliczymy każdą złotówkę. I nie będziemy czytać, że pieniądze przez przypadek trafiły na konto jakiegoś radnego PiS-u, który nagle zaczął handlować czy to maseczkami, czy płynem do dezynfekcji, czy respiratorami. Dziękuję, pani poseł. Proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wstępie mam prośbę, ogromną prośbę do pana prezydenta oraz pana premiera, aby nie wprowadzali opinii publicznej w błąd. Wszyscy wiemy, że granie na emocjach ludzi w czasie epidemii może być bardzo niebezpieczne. Sianie fake newsów w czasach epidemii jest szkodliwe, ale kiedy robi to premier lub prezydent państwa, jest to po prostu karygodne. Panie Premierze! Przestańcie okłamywać własnych obywateli. W kółko powtarzacie, że Unia nie pomaga Polsce w walce z epidemią i kryzysem. To wierutne kłamstwo. Przecież właśnie pracujemy nad ustawą o rozdysponowaniu olbrzymich środków finansowych, które Unia dała nam na walkę z epidemią i kryzysem. Panie Prezydencie! Panie Premierze! Nie mierzcie innych swoją miarą. To, że wy kierujecie się tylko i wyłącznie własnym partyjnym interesem, nie znaczy, że inni nie kierują się wartościami wspólnoty i solidarności. To, że wy się w kółko obrażacie i z nikim w Unii nie potraficie się dogadać, nie znaczy, że Unia zostawi nas samych w potrzebie, chyba że sami tę pomoc odrzucimy, tak jak to było w przypadku unijnego przetargu na sprzęt ochronny m.in. dla służby zdrowia. Dziś w wielu szpitalach i jednostkach służby zdrowia brakuje olbrzymiej ilości sprzętu i wyposażenia: maseczek ochronnych, kombinezonów, respiratorów itd. Dlaczego? Bo byliśmy jedynym krajem, który nie wziął udziału we wspólnym przetargu dla całej Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo rząd premiera Morawieckiego spóźnił się z dokumentami. Teraz ten sam premier Morawiecki twierdzi, że Unia Europejska nie dała jeszcze ani eurocenta na walkę z wirusem. Otóż otworzę wam oczy. Polska jest i będzie największym beneficjentem unijnych funduszy spójności przeznaczonych na walkę ze skutkami epidemii. Cieszy mnie, że ta olbrzymia pomoc trafi do samorządów, bo to one właśnie są na pierwszej linii walki z epidemią, to one są najbardziej obciążone kosztami walki z kryzysem, a państwo im w tym nie pomaga. Nie potraficie chronić swoich obywateli przed kryzysem. Przygotowaliście fatalne rozwiązania i odrzuciliście wszystkie poprawki opozycji, w tym 200 poprawek Lewicy, ale winnych szukacie wszędzie dookoła, w opozycji i w Unii Europejskiej. A może, panie premierze, czas spojrzeć w lustro? Tam zobaczy pan winnego. Winnego tego, że pół miliona obywateli straciło już pracę, kilkadziesiąt tysięcy firm zawiesiło działalność albo po prostu zbankrutowało. Według szacunków w kwietniu pracę może stracić blisko 3 mln Polek i Polaków, a każdy dzień zwłoki to 100 tys. kolejnych zwolnionych osób. A czym zajmuje się dzisiaj rząd? Grzebaniem i manipulacją w prawie wyborczym. Lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny, toczą w tej chwili heroiczną walkę z postępującą epidemią. Są zmęczeni, brakuje im podstawowych środków. Gdzie jest rząd? Rząd w Sejmie odrzuca wsparcie dla szpitali. Dlaczego? Bo projekt złożyła Lewica. Wczoraj mieliśmy do czynienia z najgorszym do tej pory dniem od początku pandemii. Zachorowało blisko 400 osób. Dziś nie dzielimy się na lewicę i prawicę, dziś różni nas to, co jest dla nas najważniejsze. Dla was to wybory i prezydent z koperty, kopertowy prezydent, a dla Lewicy liczą się miliony Polek i Polaków, liczy się los tych ludzi, którzy każdego dnia walczą o przetrwanie. I właśnie dlatego poprzemy tę ustawę, bo nie kierujemy się kluczem partyjnym, tylko wspólnym interesem obywateli, samorządów i państwa. Jednocześnie będziemy zgłaszać poprawki i patrzeć wam na ręce, aby wsparcie trafiało tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, gdzie będzie w najbardziej transparentny sposób wykorzystane.

Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani marszałek, w imieniu Koalicji Polskiej. Sytuacja jest coraz bardziej poważna. Wczoraj mieliśmy najwięcej zachorowań od momentu, kiedy rozpoznano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce.

Nie ma wciąż sprzętu ochrony dla pracowników, którzy pracują i walczą na pierwszej linii. To jest sprawa numer jeden, to jest kwestia najpilniejszego działania. Nie ma co zwlekać. Trzeba wprowadzać rozwiązania, które pomogą tym, którzy ratują zdrowie i życie, którzy pracują w sklepach, pracują w miejscach, które świadczą usługi, które są jeszcze dzisiaj dostępne.

Coraz więcej firm nie ma płynności. Nie przyjęliście, szanowni państwo z PiS-u, naszych propozycji dotyczących funduszu płynności w Banku Gospodarstwa Krajowego, które gwarantują, dają szansę na wypłaty, zakup towaru i podtrzymanie produkcji. Ona dzisiaj powinna być rozpatrywana. Kolejna sprawa to zwolnienie z PIT-u, CIT-u i ZUS-u dla wszystkich, niezależnie od wielkości firmy. Bez tego nie utrzymamy miejsc pracy. Nie ma dzisiaj miejsca na brak solidarności. Jeżeli dalej będziemy się kierować tylko i wyłącznie partykularnym interesem w dyskusji o tym, w jaki sposób, gdzie i co robić, a nie kiedy to zrobić, jeżeli będziemy odwlekać ważne decyzje, to nic z tego nie będzie. Musi być wprowadzony pakiet rozwiązań dla rolników, dla tych, którzy żywią w tak trudnym czasie. Naprawdę są zagrożone miejsca pracy w każdym obszarze naszego funkcjonowania. Bardzo ważne jest wsparcie dla samorządów.

To nie termin wyborów jest dzisiaj dla Polaków rzeczą istotną. Najistotniejszą rzeczą jest ich zdrowie i życie, miejsce pracy, to, czy w rodzinie będzie zapewnione bezpieczeństwo, i bezpieczeństwo zdrowotne, i bezpieczeństwo socjalne. Ludzie się tym martwią, o tym rozmawiają w domach.

Potrzebne są te rozwiązania, które są zawarte w pakcie, prawdziwym pakcie antykryzysowym, prawdziwej tarczy antykryzysowej, którą zaprezentowaliśmy. Dziękuję.

Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Premierze!

Nie możemy też pozwolić na to, szanowni państwo, aby nie było konsultacji z samorządowcami, z marszałkami województw, żebyśmy to pomijali, też taką propozycję przedstawiamy, jak również na to, by tam, gdzie z przyczyn niezawinionych przez beneficjenta, a wywołanych właśnie chorobą, Skarb Państwa nie był za to odpowiedzialny i nie pomagał w rozwiązywaniu tych problemów. Szanowni państwo, wnioskujemy o wydłużenie terminów. Jeśli chodzi o wnioski o płatność, proponujemy, żeby to nie było 30, ale 60 dni. Jeśli chodzi o zakończenie realizacji, proponujemy 180 dni.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Proszę państwa, to wszystko, co Unia da, to jest pół dnia pracy naszej potężnej polskiej gospodarki, którą mordujecie. Wasza tarcza to mordowanie gospodarki.

Jest to ogromna szansa dla gospodarki.

Jest wielka szansa, żeby polski przemysł zajął to miejsce. Dziękuję za uwagę. Proszę się liczyć ze słowami. Pani Marszałek! Panie Premierze! Przed Polską są wielkie wyzwania, a to, co robicie, woła o pomstę do nieba. Gospodarka się wali, wchodzimy w kryzys. Dziesiątki procent firm tracą w tej chwili płynność finansową, tysiące przedsiębiorców zawiesiło swoją działalność, setki tysięcy ludzi już zwolniono albo grozi im zwolnienie, mają redukowane wynagrodzenia. To, co zaproponowaliście, panie premierze, to tarcza biurokratyczna. Betonowe koło ratunkowe rzucone przedsiębiorcom. Dobre rozwiązania podpowiadaliśmy, ale nie chcecie słuchać. Ułatwienia, a nie nowe regulacje. Niestety, te rozwiązania zostały odrzucone, utknęły gdzieś na niskim szczeblu profesjonalistów, którzy próbowali doradzać rządowi. Nic z tego nie wyszło. Zajmujecie się tylko wyborami, zajmujecie się sami sobą. Rozgrywki w obozie rządzącym. Prezydent naciska na ministra, prezes naciska na wicepremiera, wicepremier negocjuje z premierem. Polacy się boją, Polacy umierają, bo są chorzy, bo ochrona zdrowia jest niewydolna, a wy zajmujecie się bez końca sobą. Jesteście zaślepieni swoimi partyjnymi interesami. Tak dłużej nie można. Nie tego oczekiwali Polacy, kiedy was wybierali. Dziś obserwują to, co robicie, i wyciągają wnioski. Uważacie, że zyskacie politycznie, przeprowadzając wybory w czasie epidemii. To cyniczna kalkulacja, panie prezesie. Wiecie o tym dobrze. Uważacie, że teraz jest jeszcze szansa wygrać wybory, bo kiedy będziecie z nimi zwlekać, wprowadzając normalnie, konstytucyjnie, wbrew temu, co dziś rano w radiu pan mówił, stan nadzwyczajny, wówczas ludzie dostrzegą kryzys i moglibyście przegrać. Ale może wystarczy odrobina przyzwoitości, może wystarczy odrobina ostrożności, może wystarczy odrobina rozsądku, słuchania tego, czego naprawdę chcą Polacy, a nie tego, czego chcą wasi posłowie, wasze zaplecze w spółkach Skarbu Państwa, wasi zdezorientowani urzędnicy w kancelarii premiera, wasi ministrowie i wiceministrowie, którzy dziś boją się o posady, którzy mają od was gwarancję wynagrodzeń, nie tak jak zwykli Polacy, którzy pracują w normalnych firmach, gdzie nastąpiło załamanie obrotu w wyniku waszych decyzji, którego nie rekompensujecie, ponieważ odmawiacie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, który wymuszałby urzędowe rekompensaty. Ludzie widzą, co robicie. Ludzie nie są głupi. Uważacie, że możecie bez końca manipulować zarówno przepisami konstytucji, jak i procesem wyborczym, zmieniać wszystko jak w kalejdoskopie, co 3 dni przedstawiać nowy projekt, jak to ma działać. Szanowni Państwo! Zobaczymy, co jeszcze nas czeka, czym zechcecie nas zaskoczyć. To, co robicie, to jest działanie na szkodę narodu. Dziękuję, panie pośle.

Proszę.

Panie Premierze! Słuchałem tych wypowiedzi, które akurat z tą ustawą nie miały nic wspólnego. Spróbuję odnieść się do tej ustawy.

Mam pytanie do pana premiera czy do pani minister, bo ta ustawa, jeśli dobrze czytam i rozumiem, pozwala nam na przesuwanie tych pieniędzy, które już mamy.

Po prostu ta ustawa pozwala nam na wykorzystanie jeszcze tych środków finansowych (Dzwonek), które nie zostały zakontraktowane lub nie będą wykorzystane z innych względów, na walkę z koronawirusem. Proszę o potwierdzenie tego przez pana premiera lub panią minister. Dziękuję, panie pośle. Proszę bardzo, pani poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Od kilku tygodni mówię, apeluję, mówią o tym wszyscy, że brakuje testów, brakuje środków bezpieczeństwa, ochrony dla lekarzy, dla pracowników ochrony zdrowia. W Polsce co szósty zakażony jest pracownikiem ochrony zdrowia, we Włoszech co dziesiąty. To znaczy, że tego sprzętu jest za mało i te zapewnienia, które ciągle nam przedstawiacie, że wszystko jest w porządku, są nieprawdziwe. Mam nadzieję, że z tych pieniędzy, z tych środków będą wreszcie zakupione odpowiednie ilości testów, maseczek, żeby rzeczywiście cyklicznie osoby pracujące w ochronie zdrowia mogły być kontrolowane. To jest strasznie ważne. Nie można mówić, że testów robimy dużo, bo ich nie robimy. Chciałabym wiedzieć, że każda osoba pracująca w ochronie zdrowia jest cyklicznie badana, żeby miała poczucie bezpieczeństwa. Jest to bardzo ważne, żeby takie zabezpieczenie było nie tylko w szpitalach zakaźnych, tych jednoimiennych, ale także we wszystkich innych, bo tak samo ważne są szpitale powiatowe, gdzie trafiają pacjenci. Tam także musi być zabezpieczenie.

Czy nie usłyszymy za chwilę, że trzeba ją nowelizować?

Jakie były rzeczywiste powody nieprzystąpienia Polski do pierwszego zbiorczego przetargu unijnego na zakup środków ochrony przed koronawirusem? Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Pewnie wielu zastanawia się, na co nam jest specustawa funduszowa, skoro z Unii Europejskiej nie dostaliśmy nawet złotówki. Ta ustawa jest potrzebna, byśmy mogli wykorzystać wszystkie fundusze europejskie na walkę z niebezpiecznym wirusem.

Jak wiadomo, przy dużym wsparciu posłów Platformy Obywatelskiej i Europejskiej Partii Ludowej Unia Europejska przeznaczy dodatkowo 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy i przedsiębiorstw oraz 3 mld euro na wsparcie w stanach nadzwyczajnych. Te fundusze pójdą m.in. na zakup sprzętu i środków ochrony dla sektora zdrowia. I dlatego ta ustawa jest nam bardzo potrzebna.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Natomiast to, co jest teraz najbardziej potrzebne przedsiębiorcom, to mapa wyjścia z kryzysu. Przedsiębiorcy, żeby mogli działać, podejmować decyzje, muszą wiedzieć, co będzie za miesiąc czy za 2 miesiące. Jak powiedział wybitny ekonomista Ludwig von Mises, podstawą ludzkiego działania jest planowanie.

Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziwię się, że kiedy Polacy chorują i umierają, obóz władzy dalej rozprawia o wyborach. To świadectwo z czarnym paskiem z moralności rządu i jego zaplecza.

Dzisiaj żądam, aby rząd zajął się realną pomocą, a nie wyborczymi układankami, choćby uwolnieniem firm od VAT-u. Ten projekt ustawy, choć idzie w dobrym kierunku, zwalnia jednak ludzi władzy z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W jaki sposób ministerstwo zagwarantuje uczciwość, konkurencyjność i to, aby środki unijne rzeczywiście były przeznaczane na ratowanie Polaków, a nie trafiały do kieszeni ludzi powiązanych z władzą?

Zapraszam do udzielenia odpowiedzi ministra funduszy i polityki regionalnej panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak. Bardzo proszę, pani minister.

Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za te słowa dotyczące naszej ustawy. Z tego miejsca chcę jeszcze raz powiedzieć, że Unia Europejska nie dała żadnych nowych pieniędzy na walkę z koronawirusem. To, o czym mówimy, czyli 7,5 mld euro, to są ciągle pieniądze, które są dla nas przeznaczone, dla naszego kraju, w ramach polityki spójności. Dopiero wczoraj po wielu zgłoszeniach zarówno naszego kraju, jak i innych państw członkowskich Komisja podeszła do tego bardzo poważnie i pozwoliła na uelastycznienie systemu wydatkowania środków, tak żebyśmy mogli przekierować je właśnie na walkę z koronawirusem. Dzisiaj rozmawiamy o znacznie bardziej uproszczonych zasadach wydatkowania tych środków.

Polska w roku 2019 nie zwróciła żadnych pieniędzy w ramach przeglądu śródokresowego, w ramach zasady n+3, tak jak miało to miejsce w przypadku Słowacji, Włoch, Francji czy Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo!

Regionalne programy zarządzają dzisiaj 40% alokacji, jeżeli mówimy o środkach, które są w ramach perspektywy polityki spójności. Jeżeli chodzi o to, czy ustawa zawęża zakres tylko i wyłącznie do wsparcia czy zapobiegania.

Ustawa była konsultowana z marszałkami województw, została skonsultowana i niektóre z propozycji przedstawionych przez marszałków zostały do ustawy wprowadzone. Oczywiście dajemy możliwość wydłużenia terminów zarówno na złożenie wniosku o płatność, jak i na zakończenie realizacji projektów. Ta ustawa na to pozwala.

Tak, w ramach realizacji procedowanej dzisiaj ustawy będzie można kupować sprzęt ochrony osobistej, maseczki, respiratory, i właśnie do tego potrzebne są te zliberalizowane zasady udzielania pomocy.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z przystąpieniem do przetargu na zakup, do ogólnego przetargu unijnego, to, proszę państwa, chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że pierwszy unijny zakup środków ochrony został zrealizowany na podstawie wcześniejszych zasad, a Polska nie przystąpiła do tego przetargu ze względu na decyzje, które były podjęte za czasów rządu PO-PSL.

Tak że Polska będzie realizować duży unijny przetarg. Dziękuję, pani minister. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Ogłaszam przerwę w obradach do godz. 17.30.

Wznawiam obrady. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 315-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Wysoka Izbo!

Żądamy, żeby dzisiaj mówić o Polakach, o tym, że tracą miejsca pracy, o tym, że będą likwidowane firmy. Czas wziąć się, szanowni państwo, nie za wybory, ale za pracę. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy państwa rozliczać z każdego miesiąca obowiązywania tego stanu.

W tej sprawie nie będę go zwoływała, bo przed chwileczką o tym na zebraniu Konwentu rozmawialiśmy, panie pośle.

Szanowna Pani Marszałek! Chciałbym prosić o formalne stwierdzenie, czy ta tutaj naradka mała, na którą pani kiwała, wyszedłszy w to miejsce, przyzywając członków Prezydium, to było Prezydium Sejmu czy też Konwent Seniorów. Jeśli to był Konwent Seniorów, to rad bym wiedzieć, dlaczego nie był przyzywany przedstawiciel koła Konfederacja i dlaczego w trybie tak nieoficjalnym dowiadujemy się, kiedy Sejm będzie kontynuował prace: czy jutro, czy w poniedziałek.

W żal nie wierzę, panie pośle. Nie była to żadna naradka.

Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych dotyczące rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Sejm na 9. posiedzeniu w dniu 3 kwietnia tego roku zgodnie z regulaminem Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 315 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Tych poprawek zgłoszono 13.

W trakcie dyskusji i głosowań tych 13 poprawek.

I taki jest wniosek Komisji Finansów Publicznych, żeby Wysoki Sejm wszystkie te poprawki odrzucił. Dziękuję, panie pośle. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 315. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Z poprawką tą łączy się poprawka 2. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. i 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 7. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Pani poseł, ja panią bardzo proszę, co to ma być w ogóle? Co to ma być, pani poseł, jakieś osobiste wycieczki? Proszę zachowywać się tak, jak poseł na sali sejmowej powinien się zachowywać. A jeżeli pani nie chce być na sali plenarnej, może pani następnym razem nie być.

Bardzo proszę o zaprzestanie tych dyskusji.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

A nie, przepraszam bardzo.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Mamy po raz pierwszy 460 osób. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tutaj, na tej sali, padły pytania o przetarg unijny, o środki, które przychodzą do nas, i sprzęt ochrony osobistej, który mógłby być w Polsce, o to, jaki jest stan zaopatrzenia w sprzęt ochrony osobistej.

12 marca częściowo ten przetarg został anulowany.

My oczywiście wzięliśmy udział w kolejnym przetargu na respiratory.

Na dzień dzisiejszy przekazaliśmy do szpitali, do podmiotów leczniczych, do innych osób 7240 tys. maseczek, 2699 tys. rękawiczek, 407 tys. l płynu do dezynfekcji, 575 tys. maseczek HEPA oraz zakupiliśmy i przyjęliśmy na stan 165 respiratorów, a ponad 1000 respiratorów jest zakontraktowanych. Ten sprzęt został rozdysponowany do 19 szpitali jednoimiennych, ponad 80 szpitali z oddziałami zakaźnymi, do ponad 500 pozostałych szpitali, do 105 z onkologią i hematologią, gdzie są najbardziej potrzebujący pacjenci, do 1585 zespołów ratownictwa medycznego, do ponad 9 tys. praktyk lekarzy POZ, gdzie nadal codziennie jest udzielanych ponad pół miliona porad, głównie porad telemedycznych, dzięki temu, że mamy lepszą informatyzację ochrony zdrowia, do 13 720 aptek, gdzie nadal ponad milion pacjentów odbiera leki, dzięki temu, że mają oni możliwość bez przychodzenia do lekarza odbierać leki na receptę, do laboratoriów, do Policji, do Straży Granicznej. Oczywiście to jest nadal ogromnie mało w stosunku do potrzeb. Ale dlatego mamy zakontraktowane kolejne 31 mln masek, 28 mln masek HEPA, 14 mln rękawiczek, 855 tys. kombinezonów i 1250 tys. gogli. To jest sprzęt, który będzie teraz sukcesywnie dostarczany i natychmiast przekazywany dalej. Pytaliście państwo też o testy. W tej chwili mamy 150 tys. testów, które są już w laboratoriach - one są fizycznie w laboratoriach polskich. Możliwości tych laboratoriów wynoszą ok. 8 tys. na dobę na dzień dzisiejszy, sukcesywnie te możliwości wzrastają. Nadal nie wykorzystujemy w pełni potencjału laboratoriów i testów, które są. Kolejne 150 tys. testów (Dzwonek) jest na terenie Polski, a 500 tys. mamy zakontraktowanych. Żebyśmy mogli zatrzymać tę epidemię, musimy mieć powyżej 50%, a nawet 60%. W związku z tym musimy robić wszystko, żeby postarać się nadal redukować poziom zakaźności - po to, żeby maksymalnie wypłaszczyć i maksymalnie ograniczyć liczbę chorych. Gdybyśmy nic nie zrobili, gdybyśmy nie wprowadzili tych drakońskich działań, na dzień dzisiejszy mielibyśmy ponad 8,5 tys. pacjentów zdiagnozowanych i zakażonych.

Dziękuję, panie ministrze.

Panie Premierze! Powtórzę pytanie, które tu zadawał parę godzin temu pan poseł Jakub Kulesza, przewodniczący koła Konfederacja. Kiedy skończycie z tym obłędnym pomysłem lockdownu, shutdownu, wyłączenia polskiej gospodarki? I pytanie do pana ministra zdrowia. Czy oprócz propagowania tych wszystkich, jak sam pan powiedział: drakońskich, a niektórzy powiedzą: absurdalnych, obostrzeń, typu zakaz wstępu do puszczy, zacznie pan wreszcie propagować testy, badania serologiczne, które pozwalają ustalić ewentualne pojawienie się przeciwciał, co byłoby certyfikatem upoważniającym do wyjścia z kwarantanny, zaopiekowania się ludźmi z grup podwyższonego ryzyka? Czemu nakręca pan psychozę, nie szukając realnego rozwiązania? Przecież wielu przedsiębiorców zamówiłoby takie badania dla swoich pracowników. Proszę. Minęło 9 godzin, odkąd powinno się rozpocząć posiedzenie Sejmu, i przyjęliśmy jedną krótką ustawę. Zamiast zajmować się tym, że w tym czasie kilkadziesiąt tysięcy osób dostało wypowiedzenia, zamiast zajmować się tym, że w tym czasie kilka tysięcy polskich przedsiębiorców złożyło wnioski o zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej, zamiast zajmować się tym, że w tym czasie kilkaset osób zgłosiło pilne zapotrzebowanie na środki medyczne, państwo straciliście te wszystkie godziny na to, by tłuc się między sobą, by dyskutować o jakichś absurdalnych rozwiązaniach, by ciągle powtarzać o absurdalnej dacie wyborów. Jesteśmy tutaj po to, by pracować. Raz jeszcze, panie premierze, wzywam do opamiętania się. Proszę wreszcie zająć się tym, do czego jesteśmy zobowiązani. Zacznijmy pracować wspólnie nad rozwiązaniami, na które czekają Polacy.

Wysoka Izbo! Dobrze, że pan minister zdrowia zabrał głos, bo to są najważniejsze tematy i tak naprawdę tematy interesujące wszystkich naszych rodaków. Mam jeszcze kilka pytań do pana ministra. Czy wszyscy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i wszyscy, którzy mają jakikolwiek związek z walką na pierwszej linii frontu, zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem?

Ostatnia kwestia (Dzwonek) dotyczy pacjentów, którzy mieli zaplanowane zabiegi. Jak jesteśmy przygotowani, żeby im pomagać: i teraz, i po zakończeniu tej fazy walki?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Choć wirus wpycha naszą gospodarkę w coraz większy chaos i zmusza do mrożenia inwestycji, ludzie tracą pracę, a firmy upadają, to budżet Unii Europejskiej jest teraz dla Polski gwarancją niezakłóconego finansowania, które również pomoże nam przetrwać ten trudny czas. Dlatego właśnie Lewica poprze tę ustawę. Tylko proszę, nie zepsujcie tego, drodzy państwo, bo mam nadzieję - i takie jest moje pytanie - że środki te będą proporcjonalnie rozdysponowane wśród samorządów - po równo, nie trafią tylko do samorządów, które są zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, pani poseł. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 315, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

454 - za, nikt nie był przeciw, 2 posłów się wstrzymało. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.